Wysoka Izbo! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 332. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki. Nad tymi propozycjami głosować będziemy w pierwszej kolejności. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek, za ten głos. W innym temacie. Wczoraj zmarł Wiktor Bater, jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, dziennikarz przez duże „D”, prawdziwy reporter, informujący o sprawach najtrudniejszych i najważniejszych, zawsze rzetelnie, laureat nagrody Grand Press, oddany swojemu fachowi. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka nr 37.

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Głosowało 460 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Mamy znowu pełną salę. W 7. poprawce wnioskodawcy proponują dodanie nowego art. 29a. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

Sejm wnioski mniejszości i poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 13. i 59., zechce nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości i poprawki 14., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości i poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania.

Sejm wniosek mniejszości i poprawkę przyjął. W 16. poprawce wnioskodawcy proponują dodanie nowego art. 62a. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 18. poprawce wnioskodawcy proponują dodanie nowego art. 64a. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawki odrzucił. W 20. poprawce wnioskodawcy proponują skreślenie art. 70. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm wnioski mniejszości odrzucił.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

W 26. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany w art. 71 pkt 10. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Nie wiem, czy posłowie wrócą, czy nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 26. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 28. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 36. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 42. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 40. i 42., zechce nacisnąć

Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosownia.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 51. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania.

się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 19. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 63. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 58. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 63. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 73. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

450 - za, 3 - przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 75. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 76. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 77. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Za chwilę przystąpimy do głosowania nad całością projektu ustawy. Proszę bardzo.

W głosowaniu nr 93 Wysoka Izba odrzuciła propozycję złożoną przez Konfederację ochrony kredytobiorców i leasingobiorców przed narzucanymi w tej chwili przez banki dodatkowymi opłatami za wakacje kredytowe, przed aneksowaniem umów na niekorzystnych zasadach, przed różnego rodzaju przemocą finansową, którą ze względu na trudną sytuację klientów i ze względu na brak regulacji chroniących konsumenta dopuszcza swoją biernością rząd. Osobiście odpowiada za to pan, panie premierze. Doskonale zna pan tę materię jako były prezes banku.

Dziękuję, panie pośle.

13 dni temu przyjmowaliśmy tarczę 1.0.

Nie przyjęliście dobrych rozwiązań, które od kilkunastu dni leżą w Wysokiej Izbie. Zwolnienie z ZUS-u przez 3 miesiące dla wszystkich, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych, 20 mld na służbę zdrowia, testy dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Zamiast tego będziemy za kilka dni obradować nad kolejnym dokumentem. W międzyczasie upadnie kilka tysięcy [[Dzwonek]] polskich podmiotów. Proszę bardzo, pan poseł Robert Kwiatkowski, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Dlaczego? Dlatego że ustawa niemal przegłosowana w tym kształcie nie spełnia kryterium dobrej legislacji. Ani ona nie jest szybka, ani ona nie jest prosta, jest pełna tzw. skutków ubocznych.

Zamiast tego forsujecie zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych dla tych, którzy handlują kryptowalutami. To jest jakieś nieporozumienie, to jest horrendum. Nie będziemy w związku z tym głosować za przyjęciem tego projektu.

Pani Marszałek! Dokładnie 2 tygodnie temu rozmawialiśmy z panią minister Emilewicz o funduszu płynności. To jest podstawowa sprawa, żeby uchronić miliony miejsc pracy przed tym, żeby były zlikwidowane, żeby Polacy utracili te miejsca pracy. Szkoda tylko, że tak późno, bo można było to przyjąć w dzisiejszych rozwiązaniach, ponieważ w prawdziwej tarczy antykryzysowej, projekcie Koalicji Polskiej, który został zgłoszony, który został rozpatrzony w pierwszym czytaniu - niestety niewiele z niego zaczerpnęliście - jest właśnie fundusz płynności. Moje pytanie brzmi: Dlaczego czekamy 2 tygodnie - teraz odczekamy kolejne dni - na to, żebyście wreszcie zrozumieli, że dobry pomysł, jeśli pochodzi od opozycji, też można przyjąć?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Mogę oczywiście wyrazić, że tak powiem, pewną przykrość, że ten projekt rzeczywiście trafił do państwa może tak późno i że nie było tak dużo czasu, który dawałby pewien komfort, ale jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji, jesteśmy w takiej sytuacji, w której potrzebujemy działać jak najszybciej. Chcemy, żeby ten projekt przeszedł całą ścieżkę legislacyjną jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy.

Dlaczego chcecie głosować przeciwko tym pomysłom? Dziś pan premier przedstawia wielki plan, wielki plan ratowania także polskich firm. Pamiętamy, że jak rządziliście, nie było nawet u szczytu waszych rządów w czasach koniunktury możliwości rozwiązania problemu głodujących dzieci. Wysoka Izbo!

Zmobilizujcie marszałka Senatu, żeby zwołał posiedzenie, żeby przyjął także projekt ustawy dotyczącej programów operacyjnych, także ten projekt ustawy jak najszybciej.

A więc jest to do zrobienia. Pokażcie swoje zaangażowanie i skuteczność w taki sposób. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 332, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wpływie interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 10. posiedzenia Sejmu, zwołanego na dni 15 i 16 kwietnia 2020 r., został paniom i panom posłom doręczony.